Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

To nie jest tak, że nic się nie stało. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której ze święta demokracji zrobiliśmy święto śmiechu. Cała Europa i świat się z nas śmieją. Nikt się nie chce przyznać do tego, że ktoś drukował karty, ktoś chciał zrealizować wybory i na dodatek jeszcze się dowiedzieliśmy, że nie było kandydatów, na koniec. Jeżeli chcemy przeprowadzić te wybory, to Lewica zaproponowała okrągły stół opozycji i koalicji, razem, nad jedną wspólną ustawą, taką, która później przejdzie przez Senat, w odpowiedzialności i w duchu porozumienia. Porozmawiajmy o tym i te obrady odłóżmy. To był pierwszy wniosek o przerwę. Ale proszę bardzo, pan poseł Jakub Kulesza. Wysoka Izbo! Chciałbym złożyć wniosek formalny nie o przerwę, ale o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji i przede wszystkim o zmianę sposobu głosowania. Za chwilę będziemy decydować o zmianie podejścia do wyborów i znosić restrykcje, ograniczenia dotyczące głosowania na miejscu. Obywatele będą mogli głosować normalnie, w lokalach wyborczych, przy urnach, a ci, co chcą, będą mogli głosować zdalnie. W związku z tą zmianą doktryny dotyczącą zwykłych obywateli wnoszę o to, apeluję do pani marszałek, żeby znieść reglamentowanie dostępu do tej sali i żeby posłowie też mieli taką możliwość: kto chce, proszę bardzo, zdalnie, ale kto chce być tu, na miejscu, bo się boi, że przez awarię sieci telekomunikacyjnej nie będzie mógł zagłosować, żeby miał możliwość zagłosowania. Doskonale pan o tym wie. Proszę bardzo, pan poseł Wojciech Saługa, Koalicja Obywatelska. Proszę. Wysoki Sejmie!

Docierają do nas coraz bardziej niepokojące informacje, wręcz alarmujące. W innych częściach kraju epidemia przygasa, natomiast na Śląsku, jak dzisiaj podano, są 204 nowe zakażenia. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jaka jest prawda, celem uspokojenia sytuacji, ponieważ w tym obiegu informacyjnym, tym szumie krąży coraz więcej niesprawdzonych, być może nieprawdziwych, informacji, chociażby ta, że zabrakło testów dla górników i nie można wszystkich przebadać. Kolejny wniosek o przerwę. Proszę. Wysoka Izbo! 12 maja 1926 r. rozpoczął się pucz wojskowy, w wyniku którego 379 osób poniosło śmierć, po obu stronach konfliktu, 1 tys. osób zostało rannych. Zamach majowy, którego ofiary nie zostały do tej pory uczczone, zamach majowy, w wyniku którego legalnie funkcjonujący rząd, na czele z premierem Witosem, i prezydent Stanisław Wojciechowski podali się do dymisji, żeby zatrzymać rozlew krwi. To są wydarzenia najtragiczniejsze w naszej historii, gdzie Polak wystąpił przeciwko Polakowi, brat przeciwko bratu, gdzie polała się bratnia krew. Niech te wydarzenia sprzed 94 lat będą dla nas wszystkich przestrogą. Uczcijmy pamięć tych, którzy zginęli, chwilą ciszy.

Dziękuję bardzo. Grupa posłów przedłożyła projekt. Proszę bardzo. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Grupa posłów przedłożyła projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, druk nr 368, wraz z autopoprawką, druk nr 368-A. Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia porządku dziennego o pierwsze czytanie tego projektu. Jest to w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu punkt sporny porządku dziennego. Propozycję uzupełnienia porządku dziennego o ten punkt poddam pod głosowanie. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przyjęcie propozycji uzupełnienia porządku dziennego oznaczać będzie, że Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, druki nr 368 i 368-A, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm propozycję przyjął. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusji nad dodanym punktem porządku dziennego. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Słyszę sprzeciw. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem propozycji Prezydium Sejmu dotyczącej wysłuchania 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 30. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druki nr 368 i 368-A) Proszę pana posła Przemysława Czarnka o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Szanowni Państwo! To nie jest tak, że chcemy przeprowadzić wybory, jak słyszałem tutaj z mównicy. Nie jest tak, że: jeżeli chcemy przeprowadzić wybory. Przeprowadzenie wyborów prezydenckich nie jest kwestią chcenia. To jest kwestia obowiązku konstytucyjnego. Kończy się kadencja urzędującego prezydenta i obowiązkiem państwa jest przeprowadzenie wyborów prezydenckich. A więc to nie jest kwestia tego, że chcemy czy nie chcemy, tutaj to nie ma nic do rzeczy. My musimy przeprowadzić wybory prezydenckie. bo państwo musi mieć prezydenta na kolejną kadencję. I dlatego właśnie, w tych szczególnych okolicznościach, w okolicznościach stanu epidemii, w okolicznościach, które doprowadziły - nie chcę teraz mówić jakich, nie czas i nie miejsce - do tego, że głosowanie w dniu 10 maja nie mogło się odbyć, i w warunkach tych przyspieszonych wyborów, bo ponowne wybory zarządzane przez marszałka Sejmu w wyniku uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z niedzieli, z 10 maja, to są wybory przyspieszone, przedkładamy Wysokiej Izbie ten właśnie projekt ustawy. Projekt jest zatem odpowiedzią na tę sytuację i przejawem odpowiedzialności za państwo, które, raz jeszcze powtarzam, musi wybrać prezydenta na kolejną kadencję, a kadencja kończy się 6 sierpnia. Projektowana ustawa umożliwia przeprowadzenie powszechnych korespondencyjnych wyborów na wniosek. Projekt przewiduje czytelne, jasne reguły, zgodne z konstytucyjnymi zasadami powszechności wyborów, bezpośredniości wyborów, tajności głosowania i równości. W wyborach, które przeprowadzone będą na podstawie przepisów zawartych w projektowanej ustawie, każdy wyborca będzie mógł zgłosić komisarzowi wyborczemu, za pośrednictwem urzędu gminy, zamiar głosowania korespondencyjnego. Każdy.

Autopoprawka ma przede wszystkim legislacyjny charakter i zawiera legislacyjne poprawki, ale ta jedna jest istotna, po to żeby osoby znajdujące się w kwarantannie i w izolacji, które wcześniej nie wiedziały, że będą w tej kwarantannie, mogły zgłosić swój zamiar głosowania korespondencyjnego również tuż przed wyborami, a zatem do 2. dnia przed dniem wyborów. Wszyscy pozostali wyborcy, którzy nie zgłoszą zamiaru głosowania korespondencyjnego, będą mogli głosować na tradycyjnych zasadach w lokalach obwodowych komisji wyborczych, tak jak to wynika z przepisów Kodeksu wyborczego. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego będzie maksymalnie uproszczone. Może się odbyć w każdej formie: ustnej, pisemnej lub elektronicznej. Wyborca głosujący korespondencyjnie otrzyma pakiet wyborczy. Pakiet zostanie wysłany przez urząd gminy. Będzie to pakiet adresowany i zostanie doręczony za pośrednictwem operatora wyznaczonego, Poczty Polskiej, ale będzie go można odebrać również osobiście w urzędzie gminy. To będzie decyzja wyborcy, który będzie zgłaszał zamiar głosowania korespondencyjnego. Wyborcy głosujący korespondencyjnie będą mieli czas najpóźniej do 2. dnia przed dniem wyborów na wrzucenie koperty zwrotnej do nadawczych skrzynek Poczty Polskiej, tych czerwonych skrzynek, które są i funkcjonują na co dzień, umieszczonych na terenie gminy. Poczta Polska opróżni te skrzynki w dniu wyborów i doręczy pakiety wyborcze właściwej obwodowej komisji wyborczej w godzinach głosowania. Wyborca będzie też mógł skorzystać z innej formy doręczenia swojego głosu - będzie mógł dostarczyć kopertę zwrotną do swojego urzędu gminy osobiście lub za pośrednictwem innej osoby.

Czytelne zasady, które jednoznacznie wychodzą naprzeciw wielu postulatom, które w ostatnich dniach słyszeliśmy, postulatom, które były wynikiem powątpiewania w możliwość przeprowadzenia wyborów na podstawie obowiązującego obecnie stanu prawnego. Dlatego ten sposób głosowania wydaje nam się najbardziej czytelny. Będą to wybory powszechne, będą to wybory bezpośrednie, będą to wybory tajne, będą to wybory równe. Te wybory, które będą ponownie zarządzone przez panią marszałek z uwagi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej, która została podjęta w niedzielę, będą wyborami przyspieszonymi.

To wszystko wpływa również na koncepcję przeprowadzenia tych koniecznych wyborów, która jest zawarta w tym projekcie ustawy. Z uwagi na fakt, że wybory będą przeprowadzone w takich okolicznościach, wnioskodawcy zdecydowali się na zaprojektowanie przepisów, zgodnie z którymi komitety wyborcze i ich kandydaci zachowują możliwość funkcjonowania i brania udziału w kolejnych wyborach, jeżeli złożone zostanie stosowne zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminach wskazanych w kalendarzu wyborczym przez marszałka Sejmu. Nie wyklucza to oczywiście możliwości kandydowania innych osób, które zgłoszą się w terminach przewidzianych w kalendarzu wyborczym, który będzie załącznikiem, który będzie przekazany równolegle z postanowieniem o zarządzeniu wyborów.

Zdaniem wnioskodawców, Wysoka Izbo, byłoby skrajną nierównością, gdyby nie dostrzeżono tego faktu, tego ogromu pracy wykonanej przez wszystkie komitety wyborcze i przez wszystkich kandydatów w ostatnich kilkunastu tygodniach, jeszcze raz to powtarzam, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej przyjdzie nam przeprowadzać wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W naszym przekonaniu zaproponowany tryb głosowania korespondencyjnego na wniosek powoduje, że te wszystkie zasady, o których mówiłem, w szczególności przywrócenie pełnej roli Państwowej Komisji Wyborczej, co było przedmiotem wielu niepokojów ze strony opozycji i innych środowisk. Przypomnę, że Państwowa Komisja Wyborcza była, jest i będzie najwyższym organem właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów. Państwowa Komisja Wyborcza utraciła tylko w przypadku wyborów z 10 maja uprawnienie do określania wzoru karty do głosowania. Natomiast w dalszym ciągu była, jest i będzie najwyższym organem właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów, o czym świadczy również uchwała podjęta przez Państwową Komisję Wyborczą 10 maja. Gdyby było tak, jak sugerowano, że Państwowa Komisja Wyborcza nie przeprowadza wyborów, nie miałaby również prawa do podejmowania tego rodzaju uchwały. Tym samym rozwiewamy wszelkie istniejące do tej pory wątpliwości i wychodzimy naprzeciw wielu postulatom zgłaszanym przez opozycję. Liczymy na współpracę po stronie opozycji, liczymy na merytoryczną dyskusję, liczymy na merytoryczne poprawki i prosimy Wysoką Izbę o przyjęcie projektowanej ustawy. Jeszcze raz powtarzam: to nie jest kwestia widzimisię kogokolwiek, to nie jest kwestia chcenia bądź niechcenia przeprowadzania wyborów. To jest kwestia świętego konstytucyjnego obowiązku państwa przeprowadzenia wyborów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kończącą się kadencją prezydenta Andrzeja Dudy, a ten koniec kadencji przypada na dzień 6 sierpnia. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Przemysław Czarnek. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pani poseł. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

do tego czasu musimy wybrać prezydenta. Zobowiązuje nas do tego konstytucja, szanowni państwo, a nie ten napis, który znacie z koszulek, z którego zostało: otua, [[Wesołość na sali]] tylko konstytucja, najwyższe źródło prawa w Polsce. Niestety zrobiliście państwo wszystko, żeby Polaków wystraszyć. A to były koperty śmierci, a to była mowa o tym, że wybory będą sfałszowane czy że będą, jak mówił np. Arłukowicz, szwindlem, że to zamach stanu - pan Hołownia, że to dyktatura itd., itd. Nie chcę już dzisiaj tych wszystkich spraw przypominać.

Jak wy sobie to wyobrażacie? Dalibyście większości parlamentarnej narzędzie, które wpisałoby się w naszą strukturę funkcjonowania państwa prawa, a nie zostało do tego wymyślone i nie zostało po to powołane. Szanowni Państwo! Mam wrażenie, że chodziłoby wam o to, żeby wykorzystać to narzędzie, żebyście potem, po miesiącu czy po kolejnym przesunięciu terminu wyborów, mogli mówić: dyktatura, nie chcą zorganizować wyborów. Przypomnę, bo przesunięcie wyborów to była wasza główna propozycja - to o rok, to o ileś tam, a to, prawda, znowu o jakieś miesiące, nie wiem, różne były propozycje - że przecież mieliście państwo na stole propozycję pana Jarosława Gowina i tę propozycję również odrzuciliście: nie, bo nie, bo nie za dwa, bo za rok, bo za miesiąc, bo za trzy. i bezpieczeństwo Polaków, czy być może chodziło o coś innego.

Udało się pokrzyżować plany Jarosława Kaczyńskiego, który chciał wybrać za was prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach kopertowych. Z tym że 3 dni później ten sam pan poseł Borys Budka mówił, że powinny się odbyć wybory prezydenckie, tego właśnie 10, bez żadnego trybu zostały one wstrzymane decyzją człowieka, który nie ma ku temu żadnych kompetencji itd.

Chcieliście wyrzucić do kosza, bo nie ta data, nie taka kampania, nie takie sondaże, być może nie taka kandydatka. Jesteśmy, szanowni państwo, odpowiedzialni. Za co? ...i naprawdę spokojnie wsłuchaliśmy się w waszą histerię, ale także w wasze postulaty, naprawdę. Wrażliwi na uwagi i na postulaty Polaków, odpowiadamy państwu tą nowelizacją, która dzisiaj została zaprezentowana. Naprawdę wsłuchaliśmy się w głosy Polaków i odpowiadamy na wasze postulaty, szanowny panie przewodniczący. Chcecie zmieniać kandydata? Mówisz, masz, można powiedzieć potocznie. Jest w tej nowelizacji taka możliwość, tak że możecie się państwo nad tym spokojnie zastanowić. W związku z tym, że, jak mówię, jak mówił również mój przedmówca, wnioskodawca, naprawdę to jest poważna sprawa i z powagą i wrażliwością w wasze postulaty się wsłuchaliśmy, to mam nadzieję, że dla dobra Polski i zgodnie z konstytucją, a nie OTUA, przystąpimy dziś do pracy, będziemy to robić wspólnie i odpowiedzialnie. Szanowna Pani Marszałek! Na podstawie art. 51 pkt 2 regulaminu Sejmu, działając w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wnoszę o przystąpienie do drugiego czytania niezwłocznie po zakończeniu pierwszego, bez odsyłania poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów [[Dzwonek]] powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, druk nr 368, do komisji. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Nie ma chyba drugiego takiego ugrupowania w Europie, jeśli nie na świecie, które potrafi zrobić taki chaos, tak namieszać, a później udawać, że wszystko jest zgodne z prawem. Wy jesteście naprawdę mistrzami świata w robieniu totalnego bałaganu. Przypomnę, że to wasz guru powiedział: Wybory odbędą się w maju i tak ma być. Bez względu na to, co mówił minister Szumowski, bez względu na to, co mówił pan premier Gowin, bez względu na to, co mówili eksperci, wy się uparliście, żeby jak najszybciej przeforsować waszego kandydata, żeby ten pałac był na zawsze wasz. To wam się nie udało z prostej przyczyny - bo jest odpowiedzialna opozycja, bo obywatele nie zgodzili się na wielką farsę i kpinę, którą zaproponowaliście. Wy dzisiaj mówicie o konstytucji? Na miłość boską, to jest ostatni akt prawny, na który wy możecie się powoływać. Wprowadziliście wybory kopertowe, które miał zorganizować pan Sasin. Dzisiaj słyszę, że Sasin pojechał na Śląsk ratować górników. Broń Boże, nie wysyłajcie go dokądkolwiek, bo on za co się zabierze, to zepsuje. Bądźcie wreszcie poważni. To, co zrobiliście, to jest kpina nie tylko z opozycji - wiemy, że nie macie dla nas szacunku - ale to jest kpina z obywateli. Mówicie dzisiaj, że trzeba przyspieszyć wybory. Jedynym konstytucyjnym prawem rządu i prawem tej większości, żeby zgodnie z konstytucją przesunąć wybory, było ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Ten stan klęski żywiołowej jest faktycznie, bo od 13 marca de facto ograniczyliście prawa obywatelskie, ludzie tracą pracę, przedsiębiorcy muszą protestować, zrobiliście nie tarczę, a pałkę na tych przedsiębiorców, a teraz nagle będziecie opowiadać, że wsłuchujecie się w głos opozycji czy obywateli. Jak wsłuchujecie się w ten głos, jeśli pani poseł mówi: Przejdźmy od razu do drugiego czytania? A dlaczego? Dlatego że znowu dzielicie Polaków na lepszych i gorszych. Tak bardzo boicie się tego, co będzie wkrótce, że chcecie jak najszybciej przeforsować te wybory. Nie wiem, czy dzisiaj będzie dymisja pana ministra Szumowskiego, czy jutro. Na Boga, ludzie wreszcie zrozumcie, że konstytucję trzeba rozumieć, a nie wyciągać ją wtedy, kiedy wam się podoba. Zrozumcie, że prezydent Rzeczypospolitej to nie ma być marionetka wybrana w fasadowych wyborach. To jest pierwszy obywatel Rzeczypospolitej i musi on mieć pełną legitymację ze strony suwerena, na którego wy się powołujecie. To, co w tej chwili proponujecie, to jest jedna wielka fikcja. Proponujecie kolejną specustawę. My położyliśmy na stole, leży u pani marszałek ustawa zmieniająca Kodeks wyborczy, bo to Kodeks wyborczy reguluje kwestie wyborcze, a nie kolejne specustawy. Znaczy, wy chcecie żyć w państwie specjalnym, gdzie rządzą służby specjalne, gdzie prawo jest specjalne. Nie, można to zrobić w sposób zgodny z konstytucją, w konsensusie, ale do tego trzeba rozumieć słowo: konsensus. I tu rozchodzimy się w dwie strony, bo wy konsensus rozumiecie w ten sposób, że wrzucacie wieczorem ustawę, której nikt nie zna, przed chwilą dorzucacie autopoprawkę i jeszcze chcecie przejść od razu do drugiego czytania. Jeżeli to jest konsensus, to ja wam gratuluję takiego poczucia. Ja rozumiem, że u was się partią inaczej zarządza, wzywa się ludzi na Nowogrodzką: dostaliście zadanie do wykonania, 28 czerwca wybory, bez względu na to, jak to będzie, ma to być. Dajcie to jeszcze panu ministrowi Sasinowi, on to najlepiej zrobi. Szanowni Państwo! Od samego początku mówiliśmy: wybory muszą być uczciwe i bezpieczne. Dziękuję pani marszałek Kidawie-Błońskiej, że jako jedyna stała twardo na tym stanowisku [[Oklaski]] i dzięki takiemu stanowisku, dzięki demokratycznej większości w Senacie, dzięki naszym klubom udało się zablokować te złe przepisy. Tak, jestem dumny, panie pośle, jestem dumny z tego, że dzięki Senatowi i dzięki odpowiedzialnej opozycji. zablokowaliśmy cyrk, który fundowaliście Polakom. Samorządy... ...zablokowaliśmy absurdalne korespondencyjne wybory, które miał zorganizować wasz kolega Sasin, który za co się nie weźmie, to zepsuje. I teraz powinniście tu powiedzieć jedno słowo: dziękuję. Powinniście podziękować, że dzięki nam jest szansa, że prezydent Rzeczypospolitej będzie miał legitymację. Ale żeby to zrobić, trzeba zmienić Kodeks wyborczy, a to, co przedłożyliście (Dzwonek), to na razie nadaje się tylko do kosza. Dziękuję, panie pośle. Stanowisko klubu parlamentarnego Lewica przedstawi pan poseł Krzysztof Śmiszek. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Zanim przejdę do oceny tego projektu ustawy - my, parlamentarzyści, choć nie ukrywam, że to powinna być praca wykonana przez większość rządzącą, jesteśmy winni społeczeństwu, suwerenowi, objaśnienie sytuacji, w której jesteśmy. A jesteśmy w najgłębszym kryzysie konstytucyjnym, instytucjonalnym i prawnym od 30 lat. Nigdy w najnowszej historii nie było takiej sytuacji. Bez względu na to, kto rządził, jakie miał poglądy polityczne, nikt nie dokonał zamachu na największą świętość demokracji, jaką są wybory. Nigdy nikomu nie przyszło do głowy, żeby to święto demokracji odrzeć ze znaczenia i je po prostu odwołać, bez żadnego trybu, bez oparcia w obowiązującym prawie. Od 2 dni wszyscy się zastanawiamy, kto odwołał te wybory, co wydarzyło się 10 maja. I oczywiście możemy przyjmować różne prawne fikcje o wyborach ogłoszonych, ale nieodbytych, możemy wczytywać się w stanowiska różnych instytucji. Jedno pozostanie z nami już na zawsze: ktoś pozbawił nas decyzji, ktoś nam zabrał wolność i ktoś zdecydował za nas. I nie chodzi o to, że wybory w czasie pandemii to wyzwanie i ryzyko. Każdy obywatel zrozumiałby decyzję i z zadowoleniem przyjąłby jasne, czytelne decyzje, poparte rzetelną, ponadpolityczną debatą o przełożeniu wyborów na bezpieczny czas. Tą cnotą jest troska. Tego zabrakło. Nie zabrakło za to brawury, nie zabrakło buty, kłamstwa i arogancji. Aż nadto mieliśmy politycznej ignorancji, bezczelności i tego, co się stało już tradycją tej Izby - przepychania ustrojowych ustaw kolanem. 10 maja doszliśmy do ściany, dalej już się nie da. Brak wyborów musi być dla nas wszystkich budzikiem i musi nas wybudzić z tego koszmaru. W niedzielę widzieliśmy klęskę partii rządzącej. Ale ten chaos i bagno prawne, w którym wszyscy jesteśmy, to także bagno, w którym pogrąża się urząd prezydenta, Rzeczpospolita i jej dobre imię. Lewica zaproponowała wyjście z tego impasu. Usiądźmy wszyscy przy okrągłym stole, wszyscy, zróbmy wszyscy jeden krok do tyłu, żeby móc zrobić dwa kroki do przodu. Tylko konsensus w tej sprawie może naprawić polityczny chaos. Przy okrągłym stole koalicja rządząca i opozycja mogą wspólnie wypracować rozwiązania, które będą społecznie akceptowalne, które odbudują zaufanie do państwa. I jako Lewica będziemy pracować nad wszystkimi projektami, które mają uporządkować sytuację prawną związaną z wyborami, ale warunkiem jest szacunek do konstytucji i wybory przygotowane i przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą. Zakończmy ten chocholi taniec. Zakończmy te polityczne igrzyska śmierci. Na horyzoncie jest coś znacznie większego niż mój czy twój interes polityczny. Tym interesem jest prawo każdego obywatela do posiadania wpływu na władze. Tym interesem jest demokracja. Zakończmy te przepychanki. Niech zwycięży najlepszy. Ale zróbmy to zgodnie z procedurami, których w tej Izbie od dawna się nie szanuje, w godny sposób, w sposób, który nie będzie nikomu dawał podstawy do kwestionowania wyniku i osiągniętego mandatu. Problemów mamy całe mnóstwo: rosnące bezrobocie, upadki firm, kolejne branże pogrążone w kryzysie, zdesperowani ludzie wychodzący na ulice w obronie swojej godności, wciąż szalejąca epidemia, pochłaniająca ofiary, niedoinwestowana służba zdrowia, która żebrze o datki na portalach społecznościowych. Kilka tygodni temu z tej mównicy sejmowej powiedziałem, że kartą wyborczą się nie najemy, karta wyborcza nie zapłaci rachunku ani za gaz, ani za prąd, ale karta wyborcza wrzucona do urny z wiarą, że przyszłość może być lepsza, że władza wyłoniona dzięki tej karcie będzie kierowała się troską, empatią i zrozumieniem, jest bezcenna, bo władza wybrana dzięki tej karcie jest władzą prawowitą, bez grzechu oszustwa i buty. Dziś przed nami wszystkimi wielki test. Lewica proponuje poprawki do tej ustawy. Złożymy je do pani marszałek z wiarą, że większość je uwzględni w myśl demokratycznej zasady, że większość rządzi, ale szanuje prawa mniejszości. Sprawmy, aby obywatele znów byli dumni z tej Izby, która pomimo ostrych sporów i walki politycznej będzie umiała w obliczu kryzysu się ze sobą porozumieć. Nieodbyte wybory 10 maja zostaną już na zawsze traumą narodową. Dziś wyjdźmy z tej Izby z poczuciem, że zrobiliśmy krok, który choć na chwilę scali naszą narodową wspólnotę. Na koniec jeszcze raz apeluję do waszej przyzwoitości, odpowiedzialności za państwo i do zdrowego rozsądku. Pani marszałek (Dzwonek), panie premierze, posłowie i posłanki koalicji rządzącej, macie większość, możecie docisnąć całą opozycję łokciem, a ustawę przepchnąć kolanem, ale możecie też wykonać krok do tyłu, usiąść z nami do stołu i wypracować konsensus w sprawie wyborów, których wynik zaakceptują wszyscy. W przeciwnym razie, ktokolwiek zwycięży w tych wyborach prezydenckich, przegramy wszyscy. Jeden dzień zwłoki zmieni niewiele. Nowe prawo wypracowane wspólnie, za którym ręka w rękę zagłosuje 460 posłów, 100 senatorów, to byłoby zwycięstwo nas wszystkich, zwycięstwo demokracji i zwycięstwo Polski. Lewica wybiera Polskę. Teraz wybór należy do was. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 przedstawi Wysokiej Izbie pan przewodniczący Władysław Kosiniak-Kamysz. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Społeczeństwa organizują swoją państwowość po to, żeby porządkować życie, żeby były pewne zasady, pewne reguły. Tak to wygląda, gdy wszystko jest poukładane. Ostatnie dni i tygodnie pokazały, jak bardzo można złymi decyzjami albo brakiem decyzji doprowadzić do rozgardiaszu, bałaganu, do sytuacji, w której organizacyjnie polskie państwo jest w ruinie. Tak często powtarzaliście hasło „Polska w ruinie” 5 lat temu, tyle że to nie była ocena rzeczywistości, tylko była to zapowiedź przyszłości. Niestety do tej przyszłości i do takiej organizacyjnej ruiny polskie państwo doprowadziliście. Takie jest poczucie wielu naszych rodaków, którzy po prostu, patrząc na wasze działania, załamują dzisiaj ręce. Trzeba wyjść do przodu. I trzeba znaleźć rozwiązanie, bo tego oczekują nasi rodacy. Tak, oczekują terminu wyborów. Tak, oczekują uczciwych zasad, możliwości bezpiecznego głosowania dla wszystkich. Dzisiaj została podjęta próba, tylko na samym wstępie próbujecie już tę próbę zniszczyć, przesyłając tę ustawę bez dyskusji do drugiego czytania.

On jeszcze kilka tygodni temu mówił, że bezpieczne wybory w lokalach mogą się odbyć za 2 lata. To czy teraz poseł Szumowski zagłosuje zgodnie z rekomendacjami ministra Szumowskiego, czy odwrotnie? Jak się zachowa? Niech przyjdzie tu i odpowie na nasze pytania. Przywróćmy funkcję kontrolną parlamentu nad rządem, bo ona została utracona i dochodzi do takich sytuacji. To ma być wszystko uznaniowe i poddawane ocenie, a później regulacji przez marszałka Sejmu. Jak będzie uznaniowe, to rodzi to coraz większe wątpliwości. Jak będzie twardo wpisane do ustawy, to wątpliwości będą mniejsze. Szukajmy rozwiązania, które to uporządkuje, a nie będzie pogłębiać rozgardiasz. Czy 14 dni to jest aż tak dużo? 3 dni? Boicie się, że nasi rodacy będą protestować, jeżeli będą mieli poczucie niesprawiedliwości? Tak, mają prawo do tego protestu, tak jak mieli prawo do protestu w wielu miejscach: pod Pałacem Prezydenckim, pod sądami, kiedy widzieli, że źle się dzieje.

Nie macie w sobie tej siły, żeby przyznać się do swojego błędu. A to zawsze powoduje, że można wyjść do przodu. W jednej kwestii muszę zgodzić się z panem posłem Czarnkiem: że państwo musi mieć prezydenta. Bo dzisiaj jest prezydent, a tak jakby go nie było. Skacze na TikToku, potrafi zarapować. ale nie jest w stanie zabrać głosu w sprawie wyborów prezydenckich w Polsce. Nawet nie potrafi zarapować, macie rację. Nie potrafi nawet zarapować, ale skacze sobie tam. Prezydent Rzeczypospolitej wybrany w wolnych, demokratycznych wyborach nie jest w stanie wyjść. Jak długo pan Andrzej Duda będzie bał się Jarosława Kaczyńskiego? Musi wreszcie chociaż na to pytanie odpowiedzieć, bo na żadne inne niestety nie potrafi. Mówię to z przykrością, przecież rywalizujemy, ale wygrał wybory uczciwie 5 lat temu i nikt tego nie neguje, natomiast dzisiaj nie jest w stanie udźwignąć tej funkcji po raz kolejny w momencie epidemii, w momencie kryzysu. To pokazuje, jak bardzo są potrzebne zmiany ustrojowe w Polsce, bo one pozwoliły na takie samowładztwo, na wdarcie się przez demokrację rządów autorytarnych. Będziemy wnosić poprawki. Aby głosowanie było jak najbezpieczniejsze, musi się odbywać przez 2 dni, bo to umożliwi korzystanie z lokali wyborczych. Ten sposób hybrydowy jest ciekawy, ale żeby był właściwy, 2 dni głosowania będą dużo lepsze, bo pozwolą na bezpieczeństwo i komisji, i tych, którzy będą przychodzić. Nie będzie tłoku, nie będzie kolejek (Dzwonek) do lokali wyborczych. Można to w ciekawy sposób rozpisać. Jesteśmy gotowi do dyskusji nad tym projektem, ale prawdziwej, merytorycznej, do współpracy. Tak, można to zrobić w normalny sposób, bo trzeba to dla Polski zrobić w normalny sposób i przywrócić Polsce normalność. Wygramy tę walkę. Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Posłowie Wnioskodawcy! Rzadko zdarza się w polityce taka sytuacja, żeby w ciągu 2 miesięcy, kiedy ktoś ma rację, wydarzenia to pokazały. 11 marca jako pierwszy kandydat w tych wyborach prezydenckich zawnioskowałem o przesunięcie terminu wyborów. Jako pierwszy powiedziałem, że będą państwo mieli problem z przeprowadzeniem wyborów, że będziecie mieli problem ze skompletowaniem komisji, że ta tradycyjna procedura w warunkach epidemii i kwarantanny po prostu nie zadziała. Utrzymywaliście jeszcze do ostatnich dni, że wszystko jest w porządku. Okazało się, że nie, wybory będą przesunięte.

Przecież zabraliście je Polakom po to, żeby Polonia nie mogła głosować, bo baliście się, że Polonia popiera nas, a nie was. Nie krytykowałem tego, co zrobiliście, waszej propozycji, powiedziałem tylko: rozszerzmy to na wszystkich Polaków. Dokładnie 5 kwietnia powiedziałem: rozszerzmy głosowanie korespondencyjne na wszystkich Polaków, którzy chcą. A wy z typowym dla waszego lidera Jarosława Kaczyńskiego uporem i przewrotnością stwierdziliście, że zrobicie przymusowe głosowanie korespondencyjne dla wszystkich. Po co?

Wszystkie prognozy ministra Szumowskiego o 2 latach poszły w kąt. Zrobicie zwykłe wybory, dokładnie tak, jak mówiliśmy, że to byłby najlepszy wariant, przyznajcie to. Przez miesiąc zwlekaliście z przyznaniem racji Konfederacji. Wczoraj przedstawiłem czteropunktowy plan, jak zrobić wybory, wybrnąć z kryzysu. Musi być termin, głosowanie osobiste, korespondencyjne, uczciwa kampania. Wasz projekt odpowiada tylko na dwa z tych wyzwań. Wprowadzacie procedurę głosowania. Czekamy na termin, czekamy też na informację o uczciwej kampanii, szczególnie w mediach publicznych. Do projektu przedstawimy siedem poprawek. Radzę szczerze: czytajcie je uważnie, bo z tego, co na razie widzimy, w tych poprawkach znajdziecie pomysły na wasze przyszłe projekty.

Wysoka Izbo!

Po raz pierwszy od 30 lat nie odbyły się wybory.

Od 2005 r. rozpętujecie histerię i uniemożliwiacie tym samym realną debatę w Polsce i osiąganie konsensusu. Szanowni Państwo!

Myślę, że to jest prorocze, proszę państwa, ponieważ Lewica, Platforma to jest tak naprawdę niechlubna przeszłość naszego państwa, jeśli chodzi o klasę polityczną, jest nieudolna teraźniejszość w postaci Prawa i Sprawiedliwości i przyszłość: Krzysztof Bosak i Konfederacja. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przechodzimy do pytań. Przypominam paniom i panom posłom, iż Prezydium Sejmu na podstawie art. 39 ust. 1 regulaminu Sejmu ustaliło w tym punkcie limit 30 pytań dla klubów według następującego parytetu: Prawo i Sprawiedliwość - 15, Koalicja Obywatelska - dziewięć, Lewica - trzy, PSL-Kukiz15 - dwa, a także jedno pytanie dla koła. Wyznaczam czas na zadanie pytania - 1 minuta.

Pytanie jest proste. Czy zdobędziecie się wreszcie na słowo „przepraszam” Czy przeprosicie Polaków za ten cyrk, który zgotowaliście? Czy przeprosicie za chaos i przede wszystkim czy przeprosicie za dziesiątki milionów złotych, które mogły być przeznaczone na służbę zdrowia, mogły być przeznaczone dla pracowników tracących pracę, dla przedsiębiorców, ale wy wydaliście je na druk pustych kart Sasina? Czy przeprosicie Polaków, że 2 miesiące okłamywaliście ich, mówiąc, że wybory się odbędą? Czy przeprosicie Polaków za to, że zamiast zajmować się największymi problemami i wyzwaniami, które są przed nami, czyli epidemią i skutkami gospodarczymi, przez 2 miesiące zajmowaliście się wyłącznie wyborami? Czy jeszcze dzisiaj na biurku prezesa Rady Ministrów wyląduje dymisja pana Sasina? To jest osoba, która odpowiada za ten chaos. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie zada pan poseł Maciej Konieczny, klub Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Umożliwienie Polakom głosowania korespondencyjnego to jest dobra rzecz nie tylko w czasie epidemii, ale w ogóle, ale dobre rzeczy nie powstają bez wysiłku. Za tym głosowaniem korespondencyjnym będzie stał ogromny wysiłek polskich listonoszy i ogromny wysiłek organizacyjny Poczty Polskiej. Chciałbym się upewnić, że ten wysiłek zostanie godnie opłacony, a cała operacja sfinansowana, bo w proponowanej ustawie próżno szukać jakiejkolwiek wzmianki o dodatkowym finansowaniu Poczty Polskiej. Stąd moje pytanie: Czy polscy listonosze mogą liczyć na to, że dostaną wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa, a ich wysiłek zostanie dobrze opłacony, dodatkowo opłacony? Czy Poczta Polska dostanie dodatkowe finansowanie na zorganizowanie tych wyborów? Czy cały proces powstaje w porozumieniu z pocztowymi związkami zawodowymi? Nie da się tego zrobić bez dodatkowych pieniędzy.

Wysoka Izbo!

Chcemy wyborów prezydenckich, po pierwsze, dlatego że kończy się kadencja obecnego prezydenta, a po drugie, dlatego że tego prezydenta trzeba w końcu wymienić. To jest naszym wspólnym zadaniem, dlatego chcemy to zrobić. Żeby te wybory były bezpieczne, potrzeba jednak modyfikacji tej ustawy.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo mnie cieszy ta sytuacja, że wreszcie dajemy obywatelom wybór. Kto nie jest pewny głosowania zdalnego, przychodzi do lokalu wyborczego. Kto się obawia o swoje zdrowie, ma możliwość zagłosowania korespondencyjnego. Rozszerzmy ten wybór. Być może są osoby, które boją się także otrzymania tego pakietu od listonosza, bo wiadomo, że na papierze wirus też może się utrzymywać. Wprowadźmy także możliwość głosowania przez Internet. Mamy profil zaufany, mamy ePUAP. Już w tych wyborach, które się odbyły, część z obywateli podpisywała ściągniętą kartę wyborczą, której formę opracował minister Sasin, podpisywała ją elektronicznie i wysyłała ją do delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dajmy obywatelom też taką możliwość. Idąc za ciosem, skoro rozmrażamy wybory, rozmroźmy gospodarkę, a zamroźmy biurokrację. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Otóż czekałem z nadzieją na ten projekt, bo liczyłem, że to będzie projekt, który będzie chciał łagodzić obyczaje i przeprowadzić uczciwe w Polsce wybory. Mówię to z dużą przykrością, że ten projekt jest jak beczka miodu, ale nie z łyżką, tylko z wiadrem dziegciu, bo ten projekt nie nadaje się do niczego.

Ale to, co zrobiliście w art. 13 i w dalszych, to jest po prostu zwykła granda legislacyjna, to jest bezprawie legislacyjne. Chcecie wprowadzić nie wiadomo jakie terminy, które marszałek może uchwalać bez żadnej kontroli. I pytam was: Czy zgodzicie się, żeby terminy czynności wyborczych były wpisane do tej ustawy, żeby wszyscy wiedzieli, na jakich zasadach grają? Te wybory według tej ustawy nie będą równe i bezpieczne, czyli nie będą demokratyczne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowni Państwo Wnioskodawcy! W uzasadnieniu omawianej ustawy powołujecie się państwo na wybory przeprowadzone w Korei Południowej. Co prawda tryb, metody i standardy, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą, przypominają bardziej standardy z Korei Północnej, ale ja nie o tym.

Moje pytanie jest proste: Dlaczego? Dlaczego w państwa ustawie brakuje przepisów o środkach ochronnych dla wszystkich wyborców? Dlaczego brakuje przepisów i nie ma ani słowa o ograniczeniu liczby wyborców w lokalu? Dlaczego nie ma ani słowa o stanowiskach, bezpiecznych stanowiskach dla członków komisji z osłonami ochronnymi w bezpiecznej odległości? W końcu dlaczego chcecie przerzucać koszty na samorządy, koszty jakichkolwiek środków ochronnych dla członków komisji? Na te wszystkie problemy odpowiadać będę poprawki zgłoszone przez klub Lewicy. Moje pytanie jest zatem proste: Czy je państwo poprzecie? Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie!

Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Mam pytanie, dlaczego po tej klęsce i kompromitacji związanej z głosowaniem kopertowym dalej brniecie w ślepą uliczkę pod nazwą: chaos wyborczy.

Rozumiem, że nie z opozycją, jakkolwiek to jest dobry obyczaj, ale chociaż z ekspertami. Dlaczego nie prowadzicie prac nad prawem wyborczym w sposób otwarty, transparentny i jasny? Przecież ta ustawa musi zyskać poparcie Senatu, który ma 30 dni na pracę nad nią. Dlaczego tam, gdzie powinniście budować zaufanie, siejecie nieufność i niepewność? Dlaczego wprowadzacie do ustawy, która miała naprawić to, co zniszczyliście, przepis, który daje marszałek Sejmu prawo do manipulowania w dowolny sposób terminami czynności wyborczych? Dziękuję bardzo. Pan poseł Wiesław Szczepański, klub Lewica. Wysoka Izbo! Pani Premier!

Dlaczego pracownik gminy może iść sam z przesyłką wyborczą, a pracownicy poczty muszą iść we dwójkę?

Czy nie będzie tak (Dzwonek), że jeżeli będziemy płacić pracownikom gminy, to oni wybiorą sobie miasto, a do kolonii, do jakiejś jednej wioski będzie z jednym pakietem musiał pędzić listonosz? Dziękuję bardzo, pani pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan poseł Czarnek reprezentujący wnioskodawców powiedział: Nie czas i nie miejsce, aby mówić o tym, co wydarzyło się 10 maja. A ja się pytam, panie pośle, kiedy jest ten czas i jakie to jest miejsce, bo nie ma lepszego miejsca do rozmowy o tym, co wydarzyło się 10 maja, niż polski parlament. Nie ma lepszego miejsca do rozmowy o waszej kompromitacji niż polski parlament. Nie ma lepszego miejsca do rozmowy o tym, jak sparaliżowaliście państwo, niż polski parlament. Nie ma lepszego miejsca do rozmowy o pakietach Sasina, o nielegalnie wydanych pieniądzach, o nielegalnych decyzjach niż polski parlament. Nie pozwoliliśmy, aby wybory ustawił Jacek Sasin i nie pozwolimy na to, aby procesem wyborczym ręcznie sterowała pani marszałek Witek. Dziękuję. Pan poseł Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! 10 maja miały się odbyć w Polsce wybory. Nie odbyły się. I dwa dni po tej dacie nadal nie wiemy, kiedy i na jakich zasadach te wybory mają się odbyć. Mamy chaos: chaos związany z pandemią, chaos związany z gospodarką, chaos konstytucyjny. Czy naprawdę cały czas uważa pan, że nie było podstaw do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej? Niech pan przyjdzie tutaj, na mównicę i ma odwagę powiedzieć: pomyliliśmy się, czego najlepszym dowodem jest to, nad czym teraz debatujemy. Nie daliście rady. Jesteście nieudolni, skompromitowaliście nasz kraj. Zajęci byliście zarabianiem na maseczkach, waszymi partyjnymi rozgrywkami, a nie tym, co jest najważniejsze. Wasza kompromitacja przejdzie do historii, a Polacy wasz rozliczą. Panie Pośle Kaczyński! Nie ma pana tutaj. Ale historia pana rozliczy (Dzwonek), bo pan jest odpowiedzialny za to, co się teraz w Polsce dzieje.

Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Ta ustawa, o której debatujemy, to ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów prezydenckich. Jakie są te szczególne zasady?

Czy tu są opisane szczególne zasady dotyczące bezpieczeństwa w lokalach wyborczych, bezpieczeństwa przesyłek kopertowych? Nie ma tutaj opisu tych szczególnych zasad. Opisano szczególne zasady ingerencji polityków rządzącej partii w proces wyborczy.

Pani poseł Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Pytanie do posłów i posłanek PiS: Kiedy skończycie te sasinaria? Mieliście szczęście wsłuchać się w nasz projekt i przyjąć część dobrych rozwiązań, a teraz marnujecie tę szansę pracy we wspólnocie i porozumieniu, nie chcąc odbyć normalnej debaty parlamentarnej. Ja już zamiast do posłów PiS, którzy mówią po prostu nieprawdę i każde ich „tak” trzeba rozumieć jako „nie”, zwrócę się do pani minister Emilewicz, bo pani przynajmniej sprawia wrażenie, że chce posłuchać. Pani minister, art. 14 jest skandaliczny. Zastępujecie ministra Sasina panią marszałek Witek. Przyjemniej to wygląda, ale nadal nie jest to PKW, a pani sama mówiła, że PKW powinno mieć pełną kontrolę nad procesem wyborczym. Dlaczego chcecie uderzyć w małe gminy? Dlaczego nie pomożecie im zorganizować bezpiecznych komisji wyborczych? To te najbiedniejsze gminy ucierpią na waszych przepisach. To wy zawaliliście wybory i pieniądze, zamiast iść na fanaberie pana Sasina, powinny iść do małych gmin. Jak wesprzecie pracowników poczty? Czy są [[Dzwonek]] dla nich dodatkowe pieniądze? Bardzo proszę. Rzeczywiście, jak słuchało się was wczoraj, pani premier, panie pośle, którzy reprezentujecie wnioskodawców, mówiliście o dialogu, o tym, że chcecie rozmawiać, że zapraszacie nas do dialogu, ale cokolwiek z tej strony się do was mówi, to kiwacie głowami i mówicie: nie.

Co to jest za ustawa, której najczęstszym zapisem jest: uchyla się zapisy Kodeksu wyborczego? Kodeks wyborczy w Polsce jest po to, żeby na podstawie kodeksu przeprowadzać wybory, a nie wprowadzać ustawy, które uchylają zapisy Kodeksu wyborczego. Jeżeli nie zejdziecie z tej drogi, to drugi raz stanie się to samo. Znowu wam się nie uda, znowu rozwalicie w Polsce wybory. Namawiamy do dialogu. Jeżeli nie będziecie oszukiwać, to jesteśmy w stanie tutaj dojść [[Dzwonek]] do porozumienia. Ale uczciwie.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! W 2014 r. parlament uchwalił nowoczesną ordynację wyborczą. W tym dokumencie zawarto możliwość głosowania korespondencyjnego w charakterze powszechnym, wpisano możliwość wcześniejszego głosowania dla osób, które bezpośrednio pobrały pakiet wyborczy i chciały go zdeponować w tygodniu poprzedzającym wybory w siedzibie gminy, wreszcie wpisano bardzo nowoczesny pakiet dla osób niepełnosprawnych. Ale w 2015 r. przyszedł PiS i PiS rozpoczął regularną walkę z tymi wszystkimi działaniami. Powiedzcie nam dzisiaj uczciwie: Jak wy się czujecie z tymi rozwiązaniami, które dzisiaj przywracacie do życia, a z nimi walczyliście? Powiedzcie nam uczciwie, dlaczego zachowywaliście się przez ostatnie lata jak małpa z brzytwą wobec świętego prawa Polaków do wolnych wyborów. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Cieszę się, że możemy dzisiaj rozmawiać o tym projekcie. Cieszę się, że udało się złożyć ten projekt. Rząd ocenia pozytywnie rozwiązania, które zostały zaproponowane. Polska potrzebuje prezydenta Rzeczypospolitej. To jest chyba fakt niekwestionowany przez nikogo w tej Izbie. Kadencja prezydenta upływa i jest potrzebny wybór prezydenta.

O tym wszystkim warto pamiętać. I teraz, Wysoka Izbo, mamy sytuację, w której państwo przedstawiacie opowieść i swoją narrację, która niestety, mam wrażenie, nie jest zgodna z rzeczywistością.

Przypomnę państwu, że to nie premier Jacek Sasin, że to Senat starał się, by przez 30 dni, jeszcze rzekomo twierdząc, że przygotowuje dobre rozwiązania, które mają poprawić ustawę. to było jedyne, co państwo byliście w stanie wymyślić i zaproponować.

Państwo mówicie o świetnych projektach, które mieliście, o świetnym prawie wyborczym, które przygotowaliście, i o rzekomo fatalnych zmianach, które były w poprzedniej kadencji. Przypomnę tylko, że także wówczas z tej mównicy krytykowaliście w sposób bezlitosny zmiany.

Łatwo to oczywiście zapisać, papier wszystko przyjmie, tylko pomysłu na to, jak to wprowadzić, zapewne też nie ma.

Pewnie pan prof. Czarnek mógłby o tym szerzej powiedzieć. Wysoka Izbo!

Jeżeli mamy sytuację, w której marszałek Sejmu ma 60 dni na rozpisanie wyborów, to oznacza to, że nie można go zmusić, by to był dokładnie 60. dzień od dnia podjęcia decyzji.

A co do stanu klęski żywiołowej to dzisiaj, gdy sami państwo apelujecie do rządu, by odmrażać gospodarkę, znosić obostrzenia, mówienie o tym, że należy wprowadzić stan klęski żywiołowej, jest naprawdę totalnym nieporozumieniem. Być może panuje stan klęski sondażowej w przypadku niektórych kandydatów, ale to jeszcze nie jest powód, by przekładać wybory w nieskończoność. Dziękuję bardzo, panie ministrze. W imieniu wnioskodawców głos zabierze pan poseł Przemysław Czarnek. Miał pan możliwość zadania pytania. Wysoka Izbo! Do większości z nich odniósł się już pan minister Łukasz Schreiber, więc nie będę tego powtarzał. Zacznę mimo wszystko od tego, co powiedział pan poseł Kierwiński. Naprawdę uważam, że dzisiaj nie jest czas i miejsce na to - i dlatego tego nie chciałem robić - żeby przypominać, kto jaką obstrukcją, jakim podpalaniem tego państwa i w jaki sposób, przy pomocy Senatu, samorządów, doprowadził do tego, że głosowanie w dniu 10 maja nie było możliwe. Wszystko jest zupełnie jasne, panie pośle.

Sędziowie jak najbardziej pasują do tej definicji, absolutnie nikt nie wyklucza sędziów. Bo rozumiem, że o to panu posłowi chodziło.

Z jednej strony słyszymy pana posła Bosaka, kandydata na prezydenta, który mówi w mediach o tym, że trzeba wprowadzić stan klęski żywiołowej, który będzie chronił wolności i prawa człowieka. A z drugiej strony słyszymy pana posła Kuleszę, który słusznie mówi o tym, że mamy odmrażać gospodarkę, odmrażać życie społeczne, odmrażać życie polityczne. Właśnie to robimy, dlatego nie ma najmniejszych podstaw do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Skończcie państwo ze stanem klęski żywiołowej. Stan epidemii obowiązuje na podstawie ustawy przez was uchwalonej i świetnie się sprawdza. Będzie to trochę trwało, ale jesteśmy przekonani, że damy radę.

Jedna rzecz, której musicie się pozbyć, bo tutaj padało to wielokrotnie z tej mównicy w ciągu zaledwie pół godziny. Państwo macie jedną chorobę. Ja nie jestem psychiatrą. Ta choroba nazywa się kaczyńskofobia. Dopóki cechuje was kaczyńskofobia.

Zresztą zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wnioski: o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania projektu ustawy, o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu oraz o skierowanie projektu ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Ogłaszam przerwę - 3 minuty. Bardzo dziękuję.

Wznawiam obrady. Sprawdzimy po przerwie kworum przed głosowaniami. Bardzo proszę wszystkich państwa posłów. Najpierw sprawdzimy kworum, panie pośle. obecnych na sali plenarnej, w innych salach i zdalnie o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu stwierdzenia kworum. Bardzo proszę.

Proszę bardzo, panie pośle. Nam naprawdę zależy na powadze. Jeżeli państwo chcecie pracować poważnie, chciałbym panią marszałek poinformować, bo może pani marszałek nie było przed przerwą, że my, pracując podczas pierwszego czytania, w trakcie tego czytania dowiedzieliśmy się o tym, że jest autopoprawka. Ona jest bardzo istotna.

Tak rozumiemy ten zapis.

Nie jesteśmy w stanie porozmawiać z ekspertami, nawet w klubie nie jesteśmy w stanie porozmawiać, a pani marszałek Gosiewska mówi, że między pierwszym a drugim czytaniem są 3 minuty przerwy. Albo rozmawiamy poważnie, dajecie nam czas na przeczytanie dokumentów i wniesienie merytorycznych uwag, albo to znowu jest fikcja. Przepraszam, pani marszałek, myślałem, że jest to zrozumiałe.

Proszę. Wysoka Izbo! Nie tyle z wnioskiem formalnym, ile z przypomnieniem i wspomnieniem. 85 lat temu odszedł do Pana Boga marszałek Józef Piłsudski, twórca polskiej niepodległości, ojciec założyciel naszej ojczyzny. Prosiłbym Wysoką Izbę o uczczenie minutą ciszy.

Do czego, panie pośle, wniosek przeciwny?

Proszę usiąść na miejscu, panie pośle. Ten wniosek poddam pod głosowanie.

Bardzo państwa proszę o to, żeby jednak na sali takich dyskusji nie prowadzić. Czekamy na wynik. No nie, panie pośle. Nie, prosiłam wszystkich państwa posłów o to samo.

Bardzo państwa proszę, dobrze?

Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 30. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. W dyskusji zgłoszono wnioski: - o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy, - o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania projektu ustawy, - o skierowanie projektu ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w drukach nr 368 i 368-A, zechce nacisnąć przycisk. wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Obecnie poddam pod głosowanie wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm skierował projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania. Kto z pań i panów posłów jest za propozycją niezwłocznego przystąpienia do drugiego czytania projektu ustawy zawartego w drukach nr 368 i 368-A, zechce nacisnąć przycisk.

Stwierdzam, że Sejm wyraził zgodę na przystąpienie niezwłoczne do drugiego czytania projektu ustawy. Proszę Państwa!

Natomiast, panie pośle, w związku z tym, że państwo zadeklarowaliście, że będziecie chcieli nad tym projektem pracować, ogłoszę teraz godzinną przerwę. Ogłaszam przerwę do godz. 15.30.

Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 30. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Szczęść Boże! Panie Marszałku! Wysoka pustawa Izbo! Skoro już tak ważne sprawy muszą być procedowane w ciągu tak niewielu godzin, to wnioskuję o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji, o wycofanie się przez Prezydium Sejmu ze złej decyzji o reglamentacji czasu wystąpień i liczby pytań parytetowo, odgórnie wyliczonych na klub, koło. Ponieważ, szanowny panie marszałku, dowiadujemy się, że nie tylko te poprawki, które są nam już znane z pobieżnej lektury, ale także jakieś nowe wrzutki szykuje nam pan superspecoberminister Szumowski, nie wiem, czy to się potwierdzi, panie pośle sprawozdawco, to radzi byśmy radzić nad tym, a nie przyjmować tylko bezkrytycznie do akceptującej wiadomości. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proponuję, aby Wysoka Izba podziękowała wspólnie pielęgniarkom i położnym za ich trud, zwłaszcza w tym bardzo ciężkim czasie, czasie epidemii, i złożyła również życzenia wszelkiej pomyślności. Proszę, aby Wysoka Izba w pozycji stojącej oklaskami podziękowała wszystkim pielęgniarkom i położnym. Mam do tego szczególną legitymację. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Nieformalny wniosek. Tak, jeden na klub, ale dzisiaj mamy szczególny dzień. 12 maja to jest dzień licznych rocznic, w tym 50. rocznicy śmierci gen. Władysława Andersa, który w 1970 r. w Londynie zmarł właśnie 12 maja. Myślę, że postaci Władysława Andersa nie trzeba przedstawiać. Wybitny dowódca, uczestnik I wojny światowej, uczestnik kampanii włoskiej i bitwy pod Monte Cassino.

Jeszcze jeden wniosek formalny. To jest wniosek o to, byśmy wspólnie zagłosowali za przerwą. zwołaniem Konwentu Seniorów i przedłożeniem Wysokiej Izbie projektu ustawy o zagwarantowaniu testów dla pracowników służby zdrowia, w tym pielęgniarzy, pielęgniarek i położnych. Nie jest sztuką rapować, nie jest sztuką bić brawo. Sztuką jest mowę przełożyć na czyny. Od kilku tygodni leży w tej Izbie projekt ustawy, która jest odpowiedzią na oczekiwania pielęgniarek, położnych i pielęgniarzy, całej służby zdrowia. Wy potraficie tylko pamiętać o nich raz w roku, jak jest ich święto. A my proponujemy ponad politycznymi podziałami: zadbajmy wspólnie o zdrowie, życie tych osób, bo one codziennie dla nas narażają swoje życie. Przyjmijmy dobry projekt ustawy, który leży w lasce marszałkowskiej. Przykre. Przystępujemy do drugiego czytania projektu ustawy.

Proszę usiąść spokojnie.

Otwieram dyskusję. Nie dostałem takiego zgłoszenia. Bardzo proszę. Szanowni Państwo! W Wysokiej Izbie dzisiaj jest taki dzień, w którym warto uczcić rocznice.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proponuję, aby Sejm w dyskusji w drugim czytaniu projektu ustawy wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm... Sprzeciw. Szanowny Panie Marszałku! Nieobecny Rządzie! Reglamentacja czasu dyskusji nad sprawą tak kluczową, istotną jak prawo wyborcze obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, próba procedowania nad tym prawem, tradycyjnie już w tej kadencji, na rympał, próba redukowania roli Sejmu, najwyższego organu władzy ustawodawczej, prawodawczej w Rzeczypospolitej, do roli fasady, dekoracji to zły trend, zły pomysł. Proszę wycofać się z tych złych, szkodliwych nie tylko doraźnie, ale też perspektywicznie rozwiązań i proszę nie reglamentować czasu dyskusji. Dziękuję.

Będą głosowania, będziemy głosować. Był sprzeciw. Proszę głosować.

Zacytujemy, oczywiście. Pani poseł, bardzo proszę. Proszę usiąść spokojnie, bo ukarzę pana karą regulaminową. Przeszkadza pan w prowadzeniu obrad. Proszę usiąść.

Mam nadzieję, że w dalszych pracach rzeczywiście będziemy mieli szansę je przeprocedować i o nich jeszcze rozmawiać i dyskutować. Klub Prawa i Sprawiedliwości również zgłasza poprawki. Panie marszałku, do końca drugiego czytania te poprawki panu złożymy. Ja natomiast, również w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, składam wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, druk nr 368, bez odsyłania do komisji. poprawek i wniosków zgłoszonych do tego projektu po doręczeniu ich posłom. Ten wniosek składam, poprawki zaraz również, do zakończenia drugiego czytania, dostarczymy. Teraz głos ma pan poseł Borys Budka, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Znaczy nic się nie zmieniło. Dalej robicie nie tylko z tej Izby, ale z całej Polski cyrk. Nie umiecie przygotować prostego projektu ustawy. Zgłaszacie go wczoraj, dzisiaj zgłaszacie autopoprawkę, w drugim czytaniu zgłaszacie jeszcze poprawki i chcecie, żeby przejść niezwłocznie do trzeciego czytania. Gratuluję takiego podejścia do dialogu. Na Boga, wy proponujecie kolejną farsę. Co więcej, wy sami nie wiecie, o co wam chodzi, bo nagle pan minister Szumowski kwestionuje ten wasz projekt ustawy. Musicie się zdecydować, czy kłamiecie wtedy, kiedy mówicie, że jest zagrożenie epidemiczne, czy kłamiecie wtedy, kiedy mówicie, że da się to zorganizować. Ja o jednej rzeczy zapomniałem przy pierwszym czytaniu. Otóż chciałem bardzo serdecznie podziękować samorządowcom, podziękować tym wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom, którzy nie przestraszyli się was, nie chcieli działać bezprawnie, bo dzięki nim, dzięki stanowczej postawie i niepoddaniu się temu dyktatowi nie wyciekły bezprawnie dane osobowe dziesiątków milionów osób w Polsce. Bo wy próbowaliście rękami Poczty Polskiej wyłudzić dane wyborców, nie mając do tego żadnej podstawy prawnej. My mówimy: sprawdzam. Chcemy z wami rozmawiać, chcemy pracować nad dobrymi rozwiązaniami w Kodeksie wyborczym, ale nie specustawą, która jest składana i uchwalana w ciągu 24 godzin, bo wy jak zawsze coś zepsujecie. Chcemy, żeby te zmiany znalazły się w prawie wyborczym, bo jesteśmy w Polsce. W Polsce obowiązuje Kodeks wyborczy, a nie specustawy. Wy chcecie całą Polskę przekształcić w stan wyjątkowy, w specpaństwo, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zgodnie z konstytucją zapewnić bezpieczne i uczciwe wybory. Wy mówicie, że to była obstrukcja, że to Senat zablokował. Nie, dobre rozmowy z Jarosławem Gowinem i to, na co się umówiliśmy, pozwoliły wyrzucić pomysł waszego prezesa, że wybory mają odbyć się w maju. Nie patrzymy na interes polityczny. My mówimy wyraźnie: wybory muszą być uczciwe i bezpieczne. Możemy ponieść najwyższą cenę, ale ważniejsze od doraźnego celu politycznego jest to, by Polacy mogli pójść do wyborów i byśmy przeprowadzili wolne i uczciwe wybory. Wy proponujecie, szanowni państwo, farsę. Proponujecie prawo pisane na kolanie, prawo nadzwyczajne, które niczego Polakom nie daje. Jutro spotykamy się podobno w gronie wszystkich klubów i kół parlamentarnych, tylko co z tego, skoro jutro mamy rozmawiać o czymś, co wy dzisiaj przyjmiecie? To nie jest forma dialogu. Zamknęliście Sejm, zrobiliście z niego farsę, a teraz jeszcze robicie farsę z ustawy, która ma sprawiać pozory legalności wyborów. Apelujemy raz jeszcze: jesteśmy gotowi na to, byśmy wspólnie przyjęli dobre rozwiązania, ale w Polsce od tego jest Kodeks wyborczy, a nie specustawy.

Wysoka Izbo! Tak jak powiedziałem kilkadziesiąt minut temu, dzisiaj jesteśmy w dniu szczególnym, ale też jesteśmy w sytuacji niezwykle szczególnej: jesteśmy pod ścianą. Wszyscy jesteśmy pod ścianą, Polska jest pod ścianą. 2 dni temu nie odbyły się wybory i nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto te wybory organizował, kto te wybory odwołał, jaki będzie dalszy los tego świętego prawa, jakie przysługuje każdemu obywatelowi i każdej obywatelce, czyli prawa głosu. Jutro rzeczywiście jest dzień, w którym będziemy mogli porozmawiać bez precedensu, można powiedzieć, w gronie i koalicji, i opozycji, o tym, w jakim miejscu jesteśmy, gdzie jesteśmy, porozmawiać o potencjalnych rozwiązaniach.

Dzisiaj słyszymy, że będzie przepychanie kolanem, drugie, trzecie czytanie. Chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Izby na kilka przepisów. Art. 20. Tego nie można pominąć milczeniem. Pan minister Sasin z panem premierem Morawieckim wydali jakieś dyspozycje bez podstawy prawnej, wydali dziesiątki milionów złotych na drukowanie kart i pakietów wyborczych i nikt nie chce wziąć za to odpowiedzialności. Ten przepis legalizuje ich bezprawie.

Chciałbym jednak zobaczyć, co w tych rozporządzeniach będzie. Komisje wyborcze trzyosobowe. To jest przecież fundamentalna zasada przeprowadzania wyborów: jawność i pluralizm w komisjach wyborczych. Mocno wątpliwe wydaje się to, że trzyosobowa komisja wyborcza będzie gwarantowała jawność, będzie gwarantowała pluralizm. Co w sytuacji gdy wszyscy będą rekomendowani z jednego komitetu wyborczego? Lewica składa szereg poprawek i od nich uzależniamy dalszą dyskusję nad tym projektem ustawy.

Wysoka Izbo! Pierwsze czytanie, które odbyło się kilka godzin temu, pokazało, że temu projektowi dosyć daleko do doskonałości, wbrew temu, co tutaj pan prof. Czarnek dowodzi. Pierwsza rzecz, panie pośle wnioskodawco.

Tu państwo zostawiacie całkowitą lukę. Panie pośle, to nie jest dobre. To po pierwsze. Jeśli, panie pośle, mówimy o tym, żeby standardy podnosić, a nie zaniżać, to wolę, żeby obligatoryjnie sędzia był członkiem okręgowej komisji wyborczej, a nie tylko mógł nim być.

To jest czerwiec, lipiec, kiedy mamy do czynienia z bardzo długim dniem.

Wysoka Izbo! Pozwolę sobie nie komentować tego, co przed chwilą wydarzyło się ze strony pana marszałka. Przejdę po prostu do konkretów, jeśli chodzi o sam projekt. Otóż Konfederacja zgłasza siedem poprawek. Są to poprawki konkretne, są to poprawki merytoryczne.

Dlatego też proponujemy, żeby wyrównać te dysproporcje. Do pakietów wyborczych, które byłyby przygotowywane, komitety wyborcze mogłyby zgłaszać, przynosić swój materiał wyborczy, którego wzór ustalałaby komisja wyborcza. To jako trzecie. Czwarta rzecz.

Środki finansowe.

Proponujemy, aby była ciągłość dotycząca wpłat, żeby nie było tej wyrwy pomiędzy 9 maja a datą zawiadomienia, które państwo proponują. Mówimy też w szóstej poprawce, że nie może być tak, aby w komisji wyborczej były tylko trzy osoby. To jest zdecydowanie za mało. Po pierwsze, bezpieczeństwo, po drugie, jakość pracy samej komisji wyborczej, po trzecie, sprawność pracy komisji wyborczej. Trzy osoby to za mało, ta praca prawdopodobnie nie będzie wykonana właściwie.

Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Braun, koło Konfederacji. Do mikrofonu zaproszę zaraz pana przewodniczącego koła Konfederacja Jakuba Kuleszę, który trzyma w ręku regulamin Sejmu. Panie Marszałku! Posuwa się pan do działań tak jawnie bezprawnych, że wypada tylko przypuszczać, że być może dało się we znaki niedotlenienie związane z tą maskaradą, którą państwo tutaj uprawialiście w ostatnich tygodniach. To jest scenariusz optymistyczny dla pana. Proszę, korepetycje z regulaminu Sejmu - pan poseł Jakub Kulesza. Szanowni Państwo! Dziękuję bardzo.

Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Marek Suski, klub Prawo i Sprawiedliwość.

Zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu i prowadzenie obrad Sejmu. Na podstawie art. 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku.

Zamykam listę zgłoszonych do pytań. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Chciałem zadać pytanie posłowi sprawozdawcy, bo rzeczywiście łatwo jest oskarżać rząd o złe intencje, jednocześnie mówiąc o tym, że głosowanie korespondencyjne jest czymś złym, i proponować klasyczne głosowanie.

Dotyczy to już funkcjonowania i samej strony technicznej działania komisji, ponieważ ci, którzy zgłosili się do udziału w komisjach. Jak będzie wyglądała ewentualnie kontynuacja? Pan poseł Marek Sowa, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przez wiele ostatnich tygodni obserwujemy nieustające próby demolowania Kodeksu wyborczego. Dzieje się to wszystko za aprobatą człowieka, który podpisuje wszystko, co mu podsuniecie. Robi to między TikTokiem a nieudolną próbą rapowania. W sobotę podpisał ustawę, która dzisiaj zostanie uchylona w całości. Czy można bardziej się skompromitować? Czy nie czujecie, że po raz kolejny upokorzyliście tego swojego prezydenta? Dlatego chciałbym zapytać, dlaczego w projekcie ustawy nie ma kalendarza wyborczego. W czwartek podpisujecie porozumienie, a w sobotę już zastanawiacie się, jak je złamać. Tacy jesteście, bo taki jest PiS oraz jego lider, którego jesteście zakładnikami.

Wysoka Izbo! Po szalonej farsie z ostatnich miesięcy związanej z organizowaniem wyborów przez PiS zaproponowaliście państwo projekt, który można określić jako ilustrację kadłubkowej demokracji. W tym projekcie proponujecie państwo, aby wieloosobowe organy zastąpić kilkuosobowymi, a nawet jednoosobowymi. Proponujecie, żeby komisje wyborcze były trzyosobowe. Proponujecie, aby zaledwie 3 dni wystarczyły na złożenie protestu do Sądu Najwyższego. I co najważniejsze, proponujecie, aby osoba, która dotychczas odpowiadała tylko za wyznaczenie daty wyborów, dzisiaj odpowiadała za wszystko. Pani marszałek Witek, która jest człowiekiem PiS, może dzisiaj zrobić wszystko według litery prawa, tej ustawy.

Pan poseł Paweł Szramka, klub Koalicji Polskiej. Bardzo proszę. Pani poseł, dziękuję. Wysoka Izbo! Zdradzę państwu, że na dzisiejszym posiedzeniu klubu poselskiego Koalicja Polska, które odbyło się przed tym posiedzeniem Sejmu, rozmawialiśmy o tym, że warto byłoby w końcu dojść do porozumienia i zamknąć tę sprawę. Natomiast widzimy, że jest to niemożliwe. To, co robi pan marszałek, jest niedopuszczalne. Tutaj - pełne wsparcie dla kolegów z Konfederacji, bo to, o czym mówicie, jest oczywiście prawdą: Pan marszałek naruszył powagę Sejmu, naruszył regulamin. Mówicie, że chcecie, ale nie robicie tego, nie odsyłacie projektu do komisji, gdzie moglibyśmy merytorycznie na ten temat porozmawiać, skracacie czas wypowiedzi posłów, tak że nawet trudno w tym czasie zadać jakiekolwiek pytania, a i tak pewnie odpowiedzi byśmy nie dostali.

Bo to, że wy to popsujecie, wszyscy wiemy. Dziękuję, panie pośle.

Pytanie do nieobecnego ministra, premiera, całej tej ekipy. Skoro przyczyny, dla których przez ostatnie tygodnie i miesiące utrzymywaliście, że nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów w trybie rutynowym, że tak powiem, w realu, z głosowaniem w lokalach wyborczych, jak rozumiem, najwyraźniej ustały, już ich nie ma, to jakie są powody, dla których życie publiczne w Polsce, przestrzeń publiczna, inne lokale, niekoniecznie wyborcze, miałyby nadal pozostać zamknięte? Jaka jest podstawa prawna i jaka jest podstawa naukowa takich decyzji administracyjnych, których kontynuacją ciągle nie waha się grozić narodowi pan minister Szumowski? Pani poseł Barbara Bartuś, klub Prawa i Sprawiedliwości. Wysoka Izbo!

Panie Pośle! Czy ten projekt ustawy zawiera mechanizmy, które uniezależniają Polskę od dalszej obstrukcji różnych środowisk, które doprowadziły do tego, że w ustawowym terminie 10 maja te wybory się nie odbyły? Czy ten projekt zawiera takie mechanizmy? Dziękuję bardzo. Pani poseł Małgorzata Tracz, klub Koalicji Obywatelskiej. Wysoka Izbo! Dziś po raz kolejny, zamiast zajmować się kryzysem gospodarczym, zdrowotnym, społecznym, zajmujemy się kryzysem konstytucyjnym, kryzysem demokracji, który wywołaliście wy, rząd Zjednoczonej Prawicy. Kryzysem, którego dałoby się uniknąć, gdybyście posłuchali głosu opozycji, która wzywała was do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej od 2 miesięcy. Ale wy woleliście w swoim zacietrzewieniu, w swojej bucie przeć do wyborów w maju. I wybraliście do tego zadania najgorszego organizatora pod słońcem - ministra Sasina. Wyborów wam nie zorganizował, po drodze kilka razy złamał prawo, wydał miliony złotych, a jedyne, co po nim zostanie, to nowy prezes Poczty Polskiej i kilka ton makulatury. Gdzie są te pakiety? 33 mln pakietów wyborczych. Kto ich teraz pilnuje? Pan poseł Dariusz Wieczorek, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jest poza dyskusją, że 10 maja miały być wybory, a tych wyborów nie było i jesteśmy. chyba jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie do takiej sytuacji doszło. To się stało. Dzisiaj na tej sali mamy po prostu problem konstytucyjny i mamy problem prawny, co dalej zrobić, i mam wrażenie, że Polki i Polacy rzeczywiście oczekują od nas, żeby jakoś ten problem rozwiązać. W związku z tym mam dwa pytania. Pierwsze pytanie: Czy rzeczywiście ten projekt ustawy konsultowaliście z Państwową Komisją Wyborczą? Bo tam jest przecież wiele rzeczy i wiele zadań dla Państwowej Komisji Wyborczej.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 2 dni po spalonej dacie wyborów, a data kolejnych wyborów jest owiana tajemnicą niczym ostrym cieniem mgły, jak powiedział klasyk. Art. 5 mówi o tym, że wszystko spoczywa na samorządach. Samorządy znowu dowiedzą się na kilka dni, na 2 dni przed datą, kiedy mają wydawać pakiety, że mają taki obowiązek. Pan minister Sasin 2 dni przed wyborami mówił, że Poczta Polska jest gotowa do przeprowadzenia wyborów. Czy dzisiaj będzie to jedynym wytłumaczeniem, jeśli znowu nie uda się przeprowadzić tych wyborów, że wrogie samorządy nie dały rady? Taka jest wasza metoda. Pan poseł mówi tu o kaczyńskofobii. Ja myślę, że takiej kaczyńskofobii nie mamy na sali tutaj.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Dużo mówiliście o Polsce w ruinie, ale widzę, że z przytupem przeszliście od słów do czynów. Bałagan, chaos i cyrk - tak należy nazwać to, co zrobiliście. Bo jak inaczej nazwać to, że dwóch szeregowych posłów spotyka się i decyduje o tym, jak zachowają się instytucje państwowe, co zrobi Sąd Najwyższy? To już nawet nie jest komedia. To jest jakiś dramat. Przez ostatnie tygodnie, zamiast zajmować się walką z kryzysem, zajmowaliście się walką o władzę, zamiast pomagać służbie zdrowia, pracownikom i pracodawcom, wydawaliście dziesiątki milionów złotych na drukowanie kart wyborczych i urny. Odpowiedzcie na pytanie: Ile milionów złotych wydaliście na przygotowanie wyborów, pseudowyborów, które nie odbyły się 10 maja? Prędzej czy później prezydent zostanie wybrany. Te głosy trzeba będzie policzyć, a potem was rozliczyć za tę niekompetencję. Pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, klub Lewicy. Wysoka Izbo! Art. 18 stanowi: W skład okręgowej komisji wyborczej wchodzi od 4 do 10 członków powołanych spośród osób mających wykształcenie wyższe prawnicze oraz dających rękojmię należytego pełnienia tej funkcji. Może dzielnicowy? Jedna osoba pójdzie na obiad, druga do toalety, zostaje jedna osoba, która będzie co?

Mamy aferę Szumowskich, mamy aferę Sasina i Morawieckiego. Przecież nie możemy w ten sposób pisać prawa. Jest koronawirus, był interes do zrobienia i trzeba tych, którzy zrobili ten interes, rozliczyć. Pan poseł Jakub Rutnicki, klub Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Ta debata trwa już kilka godzin i myślę, że wszyscy Polacy oczekują tego, żeby ktoś w końcu z PiS-u - może pan minister, który jest w tej chwili zajęty - wyszedł tutaj na mównicę i przeprosił wszystkich Polaków za tę kompromitację, jaka miała miejsce 10 maja, za te dziesiątki milionów złotych, które wydaliście nie ze swoich pieniędzy, tylko - szanowni państwo - z waszej kieszeni, bez żadnego trybu. Panie Pośle! Czy ktoś poniesie odpowiedzialność polityczną, ale także prawną za sytuację, jaka miała miejsce? Co w tej chwili przygotowujecie dla Polaków? Zamieniacie Sasina na panią marszałek Witek. Dlaczego chcecie żonglować terminami i dlaczego nie chcecie wprowadzić głosowania przez Internet? Pan poseł Konrad Frysztak, klub Koalicji Obywatelskiej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kolejny raz popełniacie błędy, a odpowiadają za to samorządy.

Ale przecież już przepaliliście przez Pocztę Polską i PWPW mnóstwo pieniędzy na karty Sasina i Morawieckiego, na urny wyborcze. O, dokładnie takie jak ta. Takie jak ta urna, która stoi w Poczcie Polskiej, a poczta twierdzi, że to nie jest jej urna. Na koniec, szanowni państwo, pytanie. Czy za wydruk kart wyborczych bez ustawy, czyli bezprawnie. odda listonosz z Wołomina, czyli Jacek Sasin, czy bankier z Wrocławia, czyli Mateusz Morawiecki?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sytuacja związana z epidemią, jak również polityczna były na tyle dynamiczne, że do ostatniego czwartku nie było pewności, że wybory się odbędą. Tymczasem odpowiedzialny za organizację wyborów minister Jacek Sasin, nie mając pewności, że wybory odbędą się w zaplanowanym terminie, uruchomił machinę związaną z drukowaniem kart do głosowania. Jego działania doprowadziły do tego, że narażono Skarb Państwa na wielomilionowe straty, a jak wiadomo, karty do głosowania to nie jest jedyny koszt. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania: Ile dokładnie kosztowały nas do tej pory wybory prezydenckie? Jaki jest koszt wydrukowania bezużytecznych kart do głosowania? Proszę również o informację, czy premier polskiego rządu zamierza wyciągnąć konsekwencje w stosunku do swojego podwładnego ministra Sasina. Pani poseł Marta Wcisło, klub Koalicji Obywatelskiej. Wysoka Izbo! Większość społeczeństwa nie chciała wyborów kopertowych, o czym mówiliśmy. Dziś zostało to nazwane histerią przez panią poseł. Przygotowaliście projekt ustawy, który ma być szczególny. Szczególny, gdyż ma dawać Polakom poczucie bezpieczeństwa i uczciwości. Ale tak nie jest, ustawa tego nie gwarantuje, o czym mówi art. 5 ust. 5. Nie, nie słyszę, pani poseł.

Co to są szczególne zasady, jeśli nie ma możliwości głosowania przez Internet? My mamy możliwość oddania zdalnie głosów, wyborcy - nie.

To jest duża sztuka, ale potrzebna. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dwa pytania. Pierwsze pytanie: Czy autorzy projektu dopuszczą możliwość zbierania podpisów poparcia dla kandydatów z wykorzystaniem elektronicznej platformy gov.pl? Wydaje mi się, że warto taką możliwość dopuścić, tym bardziej że honorujecie państwo możliwość zgłaszania elektronicznego chęci głosowania korespondencyjnego. Po co ten pośpiech? Dlaczego uchwalamy to tak na zapalenie płuc? Zmiany w prawie wyborczym muszą być wprowadzane na minimum pół roku przed wyborami - pan minister Duda, Andrzej Duda. Okres 3 miesięcy pomiędzy zmianą kodeksu a samymi wyborami jest za krótki - pan prezydent Kaczyński, Lech Kaczyński. Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz, już” - to pan prezydent Duda, tyle że z wczoraj. To się nazywa dewaluacja poglądów.

Wysoka Izbo!

Ograniczyła dyskusję i pokazała stosunek do wyborców. Ale konsekwencja. Tylko w waszym przypadku to już naprawdę nikogo nie dziwi. Problem polega na tym, że to wszystko dzieje się w sprawie wyjątkowo ważnej. Ta ustawa to fundament ustroju państwa. Ta ustawa to wiele szczegółowych rozwiązań dotyczących wyboru najważniejszej osoby w państwie w ekstremalnych warunkach, de facto w opisanym w konstytucji stanie nadzwyczajnym, którego pan premier Morawiecki cynicznie nie chce w ten sposób nazwać. A ja mam bardzo konkretne pytanie. Z kim konsultowaliście tę ustawę? Jacy uznani i wykwalifikowani prawnicy przybili stempel na waszych napisanych naprędce rozwiązaniach? Proszę o listę nazwisk, ośrodków naukowych, stowarzyszeń prawniczych. Dziękuję bardzo. Pan poseł zgłaszał się ze sprostowaniem? Pan poseł co będzie prostował? Swoją wypowiedź?

To jest nieprawda. Spędziłem tam wiele lat swojego życia i chciałbym stanąć w obronie tego miasta. Minister Sasin jest z Ząbek i chwali się tym. Teraz głos ma minister - członek Rady Ministrów pan Łukasz Schreiber. Pan życzy sobie wystąpić, panie ministrze?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dwa słowa.

Jeżeli tylko zechcą wnioskodawcy taki pomysł przedłożyć, to będzie to zrealizowane. Nie ma potrzeby, żeby obarczać samorządowców takim zadaniem, które - jak słyszymy - może rodzić jakieś trudności. Także minister zdrowia przekazał swoje rekomendacje odnośnie do projektu ustawy - nie ma w tym nic dziwnego, projekt jest projektem poselskim - po zapoznaniu się z tym przekazaliśmy także prośbę o uwzględnienie uwag ministra zdrowia.

No to jest sytuacja zupełnie kuriozalna, ale już, rozumiem, do tego się wszyscy mamy przyzwyczaić. Wysoka Izbo! Ja się zastanawiam i staram się zrozumieć, czego naprawdę część z państwa chce.

Kiedy zaproponowany został pomysł, w którym miano zabezpieczyć jak najbardziej ochronę zdrowia i życia Polaków, wybory korespondencyjne, wtedy kiedy nie wiedzieliśmy przecież, jak będzie się rozwijała pandemia, nie wiedzieliśmy, że uda się w taki sposób spłaszczyć tę krzywą zachorowań, mówiliście państwo, że to bardzo zły projekt, ponieważ teraz te wybory nie będą uczciwe. Kiedy Państwowa Komisja Wyborcza powołała się na odpowiednie zapisy, stwierdziliście, że uchwała jest zła. Kiedy teraz pojawia się na stole propozycja, tylko lepiej opracowana niż ta, którą zaproponowaliście państwo.

Ja podawałem wcześniej, jaki jest stan, mogę podać, jaki jest stan na wczoraj, bo to codziennie jest uaktualnianie.

Państwo, przynajmniej część z państwa, też pracowali nad tymi projektami i chyba nie warto tak postponować każdego działania. Tak że, Wysoka Izbo, mam nadzieję, że uda się jeszcze parę dobrych poprawek przyjąć, i naprawdę zachęcam: mniej jadu, mniej takich osobistych wycieczek, a więcej zwracania uwagi być może na konkretne zapisy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Zaczynam od odpowiedzi na pytanie czy nawet, powiedzmy, zarzuty czy wątpliwości, że żadnych odpowiedzi nie dostaniecie. Otóż mam tutaj wynotowane pytania i ustosunkuję się do nich.

Pan minister Sasin jest przede wszystkim posłem z województwa lubelskiego. Jesteśmy z tego jako mieszkańcy województwa lubelskiego bardzo dumni. Ale też chcę powiedzieć, że jest to zaproszenie pana przewodniczącego Gawkowskiego na jutrzejsze spotkanie. Z chęcią weźmiemy w nim udział, bo proces legislacyjny, tak jak tu jest napisane, trwa i trwać będzie. Proces legislacyjny składa się z prac w Sejmie, a następnie z prac w Senacie. To wszystko rzeczywiście można jeszcze bardzo ładnie pospinać. Niestety jest tak, szanowni państwo, że im dalej w las, tym więcej drzew. O ile było dosyć interesująco przy tym pierwszym czytaniu i dziękowałem za merytoryczne pytania i wypowiedzi, to w tym drugim czytaniu niestety trzeba powiedzieć, że zaczęła się już niestety tradycyjna pokazówka, aktorstwo, ale to tym bardziej nas uspokaja, bo Polacy to widzą i tego waszego aktorstwa nie mogą znieść. Merytorycznie. Merytorycznie, szanowni państwo, i o obowiązkach wobec Rzeczypospolitej Polskiej, bo po to wszyscy jesteśmy, a nie po to, żeby tu aktorstwo uprawiać na tej mównicy, bo nikt tego nie chce słuchać. Proszę państwa, najwięcej pytań i uwag merytorycznych, bo do nich się odnoszę, dotyczyło okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

Jeśli państwo dołożycie kandydatury ze swoich komitetów wyborczych, to wszędzie może być po 9 osób. Kto wam powiedział, że komisje mają być trzyosobowe?

Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło prawie 40 tys. kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Wiecie, ilu zgłosiła Platforma Obywatelska? Kilkuset. Kilkuset kandydatów i 40 tys. Jeśli państwo chcecie rzeczywiście brać udział w tych wyborach i je kontrolować, tak jak to jest zapisane w Kodeksie wyborczym - ten czynnik społeczny rzeczywiście tutaj jest - to zgłoście, na miły Bóg, kandydatów. A jak wy dalej będziecie stosować obstrukcję i nie będziecie zgłaszać kandydatów. Komisje muszą pracować.

Okręgowe komisje wyborcze.

Przecież państwo wiecie, że ten problem jest.

Dlatego wprowadziliśmy ten przepis, panie pośle, żeby w razie, gdyby doszło do tego rodzaju obstrukcji - a przecież wiemy, że dochodziło. Sędziowie pod wpływem środowiska sędziowskiego, negatywnie nastawionego do obecnej władzy, kazali tym sędziom z okręgowych komisji wyborczych podawać się do dymisji.

Taka jest rola okręgowych komisji wyborczych.

Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm przystąpił do głosowania po doręczeniu paniom i panom posłom zestawienia poprawek. Słyszę sprzeciw? Tak jest. Wobec tego do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań. Zarządzam przerwę do

Wznawiam obrady.

Bardzo proszę.

Stwierdzam kworum.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w związku z tym, że procedujemy kilka godzin w ciągu dnia nad projektem ustawy, która będzie miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, dla tego, żebyśmy polski system prawa uporządkowali i przede wszystkim przywrócili święto demokracji, które dzisiaj obróciło się w święto śmiechu. A więc gdyby udało się, pani marszałek, zarządzić przerwę, przeprowadzić jutro dodatkowe konsultacje, dokonać oceny tej sytuacji politycznej, która pozwoli później w Senacie szybkim trybem, według wzoru wszystkich partii politycznych, dojść ponad podziałami politycznymi do zgody, to wszyscy wrócimy tutaj w konsensusie politycznym. Lepiej załatwić to w polskim parlamencie, niż doprowadzić do sytuacji, w której będziemy wracali i będziemy opowiadali, że wybory są znowu źle zorganizowane. Nie zróbmy powtórki z rozrywki. Proszę w imieniu Lewicy: zróbmy przerwę i wróćmy do tego w czwartek rano.

Szczęść Boże mimo późnej pory. Wysoka Izbo!

Dajcie nam państwo szansę poprzeć niektóre z waszych autopoprawek do tego projektu, nie blokujcie ich i nade wszystko pozostańcie w zgodzie z regulaminem Sejmu, który z kolei w art. 50, pani marszałek, wyraźnie to przesądza i precyzuje, że najpierw powinny być poddane pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie przesądzi w konsekwencji o sensie głosowania nad innymi poprawkami.

Ja też mam, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zwracam się z wnioskiem formalnym o skierowanie tego projektu do komisji. Ten projekt jest projektem rangi ustrojowej, który ma fundamentalne znaczenie dla praw wyborczych w Rzeczypospolitej, dla wszystkich obywateli. Nasi poprzednicy przewidzieli rangę ustrojową dla kodeksów i specjalny tryb procedowania. Państwo oszukujecie regulamin, czyli oszukujecie samych siebie i Wysoką Izbę, udając, że to jest zwykła ustawa, a nie ustawa kodeksowa, i pracujecie nad nią kilka godzin. Ale to pokazuje, że wczoraj złożyliście wieczorem projekt, dzisiaj złożyliście kilka stron poprawek do tego projektu i jeszcze złożyliście wieczorem do drugiego czytania kilkanaście poprawek. To pokazuje, że to jest napisane na kolanie. To jest jedna wielka dziura, to jest oszustwo legislacyjne. Jeżeli tak mamy stanowić prawo w Rzeczypospolitej, prawo rangi konstytucyjnej, ustrojowej, to nisko upadła Rzeczpospolita. Przypominam, panie pośle, że podjęliśmy decyzję, że przystępujemy niezwłocznie do procedowania nad projektem ustawy. Proszę nie dyskutować.

głosowania. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 30. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Sejm przeprowadził pierwsze czytanie oraz podjął decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do drugiego czytania projektu ustawy, w trakcie którego zgłoszono poprawki. Wobec propozycji przystąpienia do głosowania po doręczeniu paniom i panom zestawienia poprawek zgłoszono sprzeciw. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przystąpienie do głosowania po doręczeniu zestawienia poprawek. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczać, że Sejm skierował projekt do komisji zgodnie ze złożonym wnioskiem. Kto z pań i panów posłów jest za przystąpieniem do głosowania po doręczeniu zestawienia poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek przyjął. Zestawienie zgłoszonych w trakcie drugiego czytania poprawek zostało paniom i panom posłom doręczone do druków nr 368 i 368-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Informuję, że łączne głosowania nad poprawkami wynikają z wniosku podmiotu je zgłaszającego.

Panie pośle, słyszał pan, że wnioskodawca decyduje o tym, czy chce zblokować poprawki, czy nie.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił.

Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Poprawka 5. stała się bezprzedmiotowa. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 14. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 16. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 18. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił.

Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 25. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 24. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 25. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 27. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. 29. poprawka stała się bezprzedmiotowa.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 36. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę odrzucił.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 39. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 40. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 44. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił.

Sejm poprawkę odrzucił. Proszę bardzo. Z wnioskiem formalnym o odroczenie posiedzenia do 14 maja. Po raz kolejny pokazaliście, że na błędach nie potraficie się uczyć. Odrzuciliście wszystkie poprawki, które miały gwarantować choć cień rzetelności przepisów, które zaprezentowaliście. Po raz kolejny pokazaliście, że nie nauczyliście się na własnych błędach, czyli proponujecie kolejną możliwość nieodbycia tych wyborów. Niestety nie wykorzystaliście szansy, żebyśmy wspólnie pracowali w Sejmie. O co? Będzie rzetelnie pracował, będzie słuchał ekspertów, [[Wesołość na sali]] wysłucha Sądu Najwyższego. Bardzo dziękuję, panie pośle, za ten wniosek. Proszę.

Jutro wszyscy się spotkamy i porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w niedzielę, a właściwie co nie wydarzyło się w niedzielę i jak wspólnie możemy naprawić to, co spotkało Rzeczpospolitą i naszych rodaków. Dzisiaj dyskutowaliśmy o ustawie ustrojowej, właściwie o ustawie, która jest jedną z najważniejszych ustaw regulujących życie społeczne. Nie można przez 2, 3 czy 4 godziny dyskutować nad tak ważnymi sprawami i przechodzić do trzeciego czytania, do głosowania nad całością.

Wysoka Izbo! Ta ustawa jest specustawą, dlatego że jest uchwalana w sytuacji absolutnie niezwyczajnej, w sytuacji, do której doprowadziła obstrukcja opozycji w Senacie. Nie prace, obstrukcja opozycji w Senacie, bo Senat nie pracował 30 dni, i obstrukcja w wielu samorządach. Dlatego jest to specustawa, bo musimy wykonać obowiązek konstytucyjny wobec państwa, przeprowadzić wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. My jutro naprawdę nie chcemy się spotykać, żeby opowiadać państwu raz jeszcze, co zrobiliście, żeby nie doprowadzić do głosowania 10 maja. Chcemy rzetelnie rozmawiać. Proces legislacyjny trwa. Jak chcecie, żeby wam powtórzyć, co zrobiliście, żeby zablokować głosowanie 10 maja, to nie liczcie na naszą długą obecność jutro na spotkaniu. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druków nr 368 i 368-A, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.